Szczęść Boże! Porządek obrad powinien być uzupełniony w trybie pilnym o nadzwyczajną informację ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego Policji zawierającą odpowiedź na pytanie, czy miasto Wrocław należy jeszcze do Rzeczypospolitej Polskiej. Doniesienia z ostatnich dni i godzin nasuwają zasadne podejrzenie, że działa się tam na podstawie jakiegoś innego prawa, prawa, które nie jest stanowione ani nie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie: Czy wszyscy państwo odebrali już karty? To jeszcze chwileczkę poczekamy, ale proszę.

Kto się wstrzymał?

Panie i Panowie Posłowie! Prezydium Sejmu przedłożyło projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, druk nr 9. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu przedłożyło wnioski w sprawie: wyboru sekretarzy Sejmu, wyboru składów osobowych komisji sejmowych, wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, a także wyboru składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej. Wnioski to odpowiednio druki nr 8, 10, 11 i 12. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych wniosków. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 9) Zgodnie z art. 137 ust. 1 regulaminu Sejmu w skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych wchodzi nie więcej niż siedmiu posłów. Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu, w drodze uchwały ustala liczbę członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, jednomyślnie proponuje, aby Sejm ustalił liczbę członków tej komisji na siedem osób. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w pierwszym czytaniu projektu uchwały?

Wysoka Izbo! Wczoraj dokonany został wstępny podział łupów, dziś ciąg dalszy. Konfederacja, rzecz jasna, zna regulamin prac Sejmu i orientuje się, jakie zasady reglamentacji obowiązują w dostępie do niektórych komisji, jednak jeszcze raz zwrócę uwagę Wysokiej Izby i czcigodnego Prezydium na fakt, że koło Konfederacji weszło do tej Izby z jednej listy, nie jest kołem składkowym. Ponieważ mówiliście tutaj państwo wczorajszego wieczora o zbrataniu, nowym otwarciu. porozumieniu ponad podziałami, bardzo nalegamy, by to porozumienie ponad podziałami nie dokonywało się ponad głowami konfederatów, [[Dzwonek]] ponad głowami 1250 tys. naszych wyborców. Prosimy o dopuszczenie do komisji do spraw spec-służb, co oczywiście wymaga zmiany regulaminu Sejmu. Dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Proponuję, aby Sejm przystąpił niezwłocznie do drugiego czytania projektu uchwały. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do drugiego czytania projektu uchwały. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu projektu uchwały? Moim pierwszym głosem dzisiejszego tak późno rozpoczętego dnia zwróciłem uwagę na to, że nie jest bezpiecznie, że nie wszyscy polscy patrioci czują się i mogą czuć się bezpieczni w Rzeczypospolitej Polskiej. ponieważ Policja państwowa na wezwanie urzędników, którzy mienią się polskimi, ale, powtórzę, nie wiadomo, na gruncie jakiego prawa operują, Policja polska dokonuje interwencji wobec polskich patriotów świętujących rocznicę niepodległości. W tym kontekście sytuacyjnym jest chyba oczywiste, że polscy patrioci, których reprezentacją jest koło Konfederacji, chcieliby trzymać rękę na pulsie rzeczywistości, mając dostęp do komisji, w której rozważa się sprawy z pewnego punktu widzenia najbardziej istotne (Dzwonek) dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 9, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 432 było za, 11 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Wybór składów osobowych komisji sejmowych (druk nr 10) Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedstawiło na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu wniosek w sprawie wyboru składów osobowych komisji sejmowych. Proszę o uwzględnienie zmiany, na prośbę Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15, w składzie Komisji Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, polegającej na wycofaniu posła Jarosława Rzepy oraz dopisaniu do jej składu posła Marka Sawickiego. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Wysoka Izbo!

Dlaczego? Ponieważ taką decyzję państwo, ponad głowami tych wyborców i posłów Konfederacji, podjęli. Żaden z posłów Konfederacji nie został dopuszczony do tych komisji. A przecież mamy dwóch posłów z Pomorza, mamy specjalistów, informatyków, specjalistów od sieci, systemów teleinformatycznych. Nie będziemy mogli brać udział w głosowaniach w tych komisjach i wyrażać woli naszych wyborców, dlatego jesteśmy przeciwko takiemu składowi osobowemu tych wszystkich komisji, dokonanemu ponad głowami Konfederacji. Dziękuję, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku. Nie miałam zgłoszenia, panie pośle. Wysoka Izbo! Otóż chciałem przypomnieć panu koledze przedmówcy, że każdy poseł może wziąć udział w posiedzeniu komisji, wypowiadać w swoim imieniu, a także wyborców, swoje racje.

Kto się wstrzymał? 437 było za, 6 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji sejmowych. Informacja w sprawie inauguracyjnych posiedzeń stałych komisji sejmowych, które odbędą się w dniu jutrzejszym, tj. 14 listopada br., dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, na podstawie art. 148a ust. 8 regulaminu Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionej propozycji?

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wyjaśnię wyborcom, że Komisja do Spraw Unii Europejskiej to jest komisja, do której spływają szerokim strumieniem tworzone przez brukselskich biurokratów prawa, często absurdalne i szkodliwe, które są narzucane Polsce często wbrew woli naszych władz. Chcielibyśmy móc brać udział w głosowaniu w Komisji do Spraw Unii Europejskiej jako przedstawiciele Konfederacji, na którą głosowało 1250 tys. wyborców. Jeżeli pan poseł uważa, że głosowanie nie jest ważne, byle móc słuchać, to proszę oddać miejsce Prawa i Sprawiedliwości, my wejdziemy na te miejsca i będziemy głosować, a państwo będą słuchać. Mowa tutaj o regulaminach, my je znamy, ale Prawo i Sprawiedliwość ma tu większość, może wszystko, nie ma ograniczeń. Wczoraj nawet posła Czarzastego uczyniła wicemarszałkiem, więc prosimy, żeby zgodnie z tym, co powiedział wczoraj Andrzej Duda, o pluralizmie i niewykluczaniu nikogo, zmienić regulamin tak, żeby Konfederacja jako koło mogła mieć pełnoprawnego członka w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Na razie obowiązuje dotychczasowy regulamin. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 11, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Głosowało 449 posłów. Za było 440, 9 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej (druk nr 12) Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedstawiło na podstawie art. 143 ust. 11 regulaminu Sejmu wniosek w sprawie wyboru Komisji Etyki Poselskiej. Przypominam, że Sejm dokonuje wyboru członków komisji w głosowaniu łącznym. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zabrać głos w tej sprawie? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 12, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? 438 było za, 10 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Wybór sekretarzy Sejmu (druk nr 8). Prezydium Sejmu na podstawie art. 6 ust. 2 regulaminu Sejmu przedstawiło wniosek w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu. Wniosek ten został paniom i panom posłom doręczony. Przypominam, że zgodnie z art. 6 regulaminu Sejmu Sejm wybiera 20 sekretarzy w głosowaniu łącznym, chyba że Sejm postanowi inaczej. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zabrać głos w sprawie zgłoszonych kandydatur?

Wysoki Sejmie! Postanowili państwo porozumieniem czterech partii politycznych, które całkowicie dominują w tej Izbie, wyeliminować Konfederację zarówno z Prezydium Sejmu, jak i z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie usprawiedliwiali to państwo niewielką liczebnością tych gremiów. Postanowili państwo wyeliminować Konfederację także z najliczniejszej komisji w Sejmie, z Komisji do Spraw Unii Europejskiej, tak żeby reprezentacja polskich eurosceptyków nie mogła nawet poprzez głosowanie pokazać, jak będzie głosowała. My się nie obrażamy, chcemy pokazać, że potrafimy służyć dobru polskiego parlamentaryzmu z każdej pozycji. Przyjmiemy tę propozycję. Nasz najmłodszy poseł, poseł z Pomorza, poseł z Gdyni, którego nie dopuszczają państwo w rozdziale miejsc w komisjach do komisji, która zajmuje się gospodarką morską, będzie nas reprezentował jako poseł sekretarz, pomagając prowadzić obrady. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku z druku nr 8, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 450 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 13 listopada br. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nikt się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Bardzo proszę, pani poseł.

Cieszę się, że na sali jest pan premier Mateusz Morawiecki, bo będę mówiła o sprawie, która wczoraj padała z tej mównicy, tj. o tym, jak to dobrze jest w ochronie zdrowia. A kilka dni temu Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ze Specjalistycznego Szpitala w Mielcu wystosowali do premiera Morawieckiego i ministra zdrowia list otwarty, apel. Apel, w którym proszą o pilne podjęcie skutecznych działań, które pozwolą powstrzymać dalszą degradację polskich szpitali, zadłużonych i zadłużających się w zatrważającym tempie. W tym liście, panie premierze, piszą do pana. Nie mamy wątpliwości, że Ministerstwo Zdrowia świadomie dąży do ograniczenia liczby szpitali, jednak metoda służąca osiągnięciu tego celu jest skrajnie nieodpowiedzialna i zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Związkowcy apelują o zajęcie się sprawą finansowania szpitali powiatowych. Ich zdaniem obecna polityka ryczałtowania szpitali wprost prowadzi do niewypłacalności tych placówek. Proszę państwa, bardzo proszę. Tych z państwa, którzy chcą prowadzić rozmowy - bardzo proszę, żeby to robić w kuluarach. Pani poseł chciałaby dokończyć swoje oświadczenie. Pani poseł, proszę. Ja doliczę pani czas. Bardzo proszę państwa posłów albo o zaprzestanie rozmów, albo o to, żeby prowadzili je w kuluarach. Raz jeszcze przypomnę, że związkowcy apelują o zajęcie się sprawą finansowania szpitali powiatowych. Ich zdaniem obecna polityka ryczałtowania szpitali wprost prowadzi do niewypłacalności tych placówek, co z kolei grozi ich zamykaniem lub prywatyzowaniem. Te opinie są odzwierciedleniem tragicznej sytuacji wszystkich szpitali, również szpitala w Mielcu. Oczekuję od rządu Rzeczypospolitej Polskiej pilnych działań prawnych i finansowych w celu oddłużenia szpitali, tak by mogły leczyć pacjentów, ponieważ z informacji samorządowców z Podkarpacia, którzy na moją prośbę informowali o sytuacji finansowej szpitali na ich terenie, wynika, że jest źle, bardzo źle. Brakuje pieniędzy na leczenie. Przykład: zła sytuacja finansowa w szpitalu miejskim w Rzeszowie, o ponad 3 mln zł na dzisiaj został przekroczony ryczałt, jaki przekazywany jest dla szpitala. Jak rozumieć więc wczorajsze wystąpienie sejmowe premiera Morawieckiego, w którym m.in. zapewnił, że zwiększyły się wydatki na ochronę zdrowia, a kolejki do lekarzy specjalistów są krótsze? To wszystko nieprawda. Kolejki są dłuższe, a finansowanie zwiększyło się dzięki wpłatom pacjentów, obywateli, którzy płacą składkę zdrowotną. Potrzebne są zatem pilne działania i zmiany, aby pacjenci mieli dostęp do leczenia. Mam nadzieję, że związkowcy z Mielca otrzymają odpowiedź na swój list otwarty, aby nie powtórzyła się sytuacja, kiedy w sprawie ceny prądu prezydent Rzeszowa przez 9 miesięcy nie otrzymał odpowiedzi. A zatem, panie i panowie posłowie, sprawa szpitali, sprawa pacjentów jest niezwykle ważna, a słowa pana premiera Morawieckiego były oczywistą nieprawdą. Związkowcy oczekują na tę odpowiedź i ja również. Dziękuję, pani poseł.